w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji: - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - bezpośrednio po zakończeniu głosowań na sali plenarnej, - Kultury i Środków Przekazu - również bezpośrednio po zakończeniu głosowań na sali plenarnej.

Proszę wszystkich o powstanie. Wysoka Izbo!

Bardzo proszę pana posła Władysława Kosiniaka-Kamysza o zabranie głosu. To prawda. Dziś rano dotarła do nas ta smutna informacja o śmierci naszego serdecznego kolegi lekarza, bo jako lekarz rozpoczynał swoją działalność społeczną, zawodową. Przez całe życie był lekarzem, wieloletnim ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala w Ciechanowie. Później był samorządowcem, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Ciechanowa od roku 1990, a następnie przewodniczącym tej rady.

Zmagał się przez wiele ostatnich lat z ciężką chorobą. Pozostawał zawsze wierny swojej małej ojczyźnie. Dla Ciechanowa, dla województwa mazowieckiego jest przykładem oddania. Cześć jego pamięci!

Proszę państwa, dzisiaj mamy też ważne daty związane ze Śląskiem. Bardzo proszę pana posła Jerzego Polaczka. Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 20 kwietnia 1873 r. urodził się Wojciech Korfanty, wielki syn ziemi śląskiej, współtwórca odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości, dyktator trzeciego powstania, którego stulecie będziemy obchodzić uroczyście w Polsce i na Górnym Śląsku za 2 tygodnie.

Bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Proszę bardzo.

Stwierdzam kworum. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1115. W związku z tym, na podstawie art. 95f regulaminu Sejmu, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, druk nr 1116. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Informuję, że po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjęłam decyzję o nieprzeprowadzaniu trzeciego czytania punktu 12. porządku dziennego, tj. sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, druki nr 1005, 1035 i 1035-A. Pan poseł Cezary Tomczyk, Koalicja Obywatelska. Proszę. Wysoka Izbo! Składam wniosek o przerwę. Wstyd! ...domniemane wykorzystanie środków publicznych na kampanię prezydencką Andrzeja Dudy oraz manipulowanie ludźmi w Internecie. Jeśli to prawda, to niczym nie różnicie się od Rosjan, którzy wpływali na wybory w Stanach Zjednoczonych. I trzeba powiedzieć to bardzo jasno: żądamy w tej sprawie jasnych wyjaśnień od prezydenta Andrzeja Dudy oraz od członków PiS-u, którzy byli w jego sztabie. Pan prezydent Andrzej Duda siedział tutaj, przysięgał przed Wysoką Izbą uczciwość. Zachodzi podejrzenie, że kampania Andrzeja Dudy była finansowana z lewych pieniędzy. 10 dni przed konkursem powstaje firma, która dostaje 40 mln zł, a później angażuje się w kampanię prezydenta Andrzeja Dudy. Wtedy kiedy cały świat zajmował się szczepionkami, wtedy kiedy cały świat zajmował się wyjściem z epidemii, wy zajmowaliście się manipulacjami. Proszę, ponieważ padł wniosek formalny o przerwę, poddam ten wniosek pod głosowanie.

Proszę to robić po cichu, dobrze? Kto z pań i panów posłów jest za ogłoszeniem przerwy, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Proszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wnoszę o przerwę i uzupełnienie porządku obrad o informację premiera w sprawie ratyfikacji tzw. Funduszu Odbudowy, a w rzeczywistości funduszu zadłużenia, i sposobu głosowania nad nim w tym parlamencie. Z informacji medialnych wynika, że rząd rozważa zastosowanie tzw. małej ratyfikacji, czyli pominięcia parlamentu. Żądamy jednoznacznej informacji, czy bez głosowania w parlamencie rząd zamierza przeforsować unijny fundusz zadłużenia i realnie nowe unijne podatki.

Był już głosowany. Proszę.

Wysoka Izbo! Składam wniosek o odroczenie posiedzenia i zwołanie Konwentu Seniorów celem uzupełnienia. punkt dotyczący zielonego zaświadczenia cyfrowego.

Dlatego bardzo proszę o to, ażeby ten punkt znalazł się również w porządku naszych obrad. Nie rozumiem, dlaczego państwo tak krzyczycie z tych ław. Padł wniosek o odroczenie, a nie o przerwę. Konwentu, pani poseł, nie zwołam, bo to jest moje uprawnienie, ale ponieważ padł wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Proszę państwa, wy tak krzyczycie, że ja w ogóle nie słyszę, co wy mówicie. Kto nie ma maseczki? Pani poseł, nie widziałam pani bez maseczki, więc uprzedzam, że jeżeli to prawda. Pani poseł, bez maseczki na salę nie wchodzimy.

W związku z tym poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.

Sejm wniosek odrzucił. Proszę. Wysoka Izbo! Zwracam się z wnioskiem formalnym o przejście do porządku obrad, ale jednocześnie rozważenie przez panią marszałek możliwości rozszerzenia tego porządku obrad. Do dnia wczorajszego prawie 6 mln sztuk drobiu zostało wybite i ta informacja ministra rolnictwa jest bardzo potrzebna. Jak wygląda przygotowanie odpowiednich służb, zabezpieczenie, wsparcie dla rolników?

Sytuacja jest bardzo trudna, wręcz dramatyczna i należałoby dzisiaj o tym podyskutować. Powracamy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1002-A. Proszę pana posła Krzysztofa Lipca o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! W imieniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka wnoszę, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić projekt ustawy zawarty w druku 1002, i jednocześnie wnoszę o odrzucenie przez Sejm wniosku o odrzucenie projektu ustawy. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1002. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości, a także w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Wnioski mniejszości od 2. do 10. zostały zgłoszone do art. 3 projektu ustawy nowelizującej, zawierającego zmiany do ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 10. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują nie wprowadzać zmian w art. 349. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1002, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1034-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę panią poseł Barbarę Bartuś o przedstawienie sprawozdania. Mam przyjemność przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W czasie drugiego czytania do projektu ustawy zgłoszono 11 poprawek i dwa wnioski o odrzucenie. Komisja Nadzwyczajna po rozpatrzeniu wniosków i poprawek na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia rekomenduje odrzucić obydwa wnioski i przyjąć osiem poprawek oraz odrzucić trzy poprawki. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1034. W dodatkowym sprawozdaniu komisja przedstawia wniosek o odrzucenie projektu ustawy oraz poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Przyjęcie wniosku o odrzucenie projektu spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy. Komisja wnosi o odrzucenie tego wniosku. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w całości projektu ustawy z druku nr 1034, zechce nacisnąć przycisk.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Z poprawką tą łączy się poprawka 11. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 3. i 11., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Poprawki od 4. do 9. zostały zgłoszone do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 5. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 8. Głosujemy.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy.

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1034, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego raz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:

Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Tomasza Ławniczaka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przedstawiam dodatkowe sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, to jest druk nr 1014, oraz senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, to jest druk nr 990. Dwie wymienione komisje na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia rozpatrzyły siedem poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu i wnoszą, aby Wysoki Sejm przyjął poprawki od 1. do 5., zaś poprawki 6. i 7. odrzucił. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1036. Komisje przedstawiają również wnioski mniejszości, a także, w dodatkowym sprawozdaniu, poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm propozycję przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1036, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powracamy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1066-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Dzień dobry państwu. Mam zaszczyt w imieniu Komisji Infrastruktury przedstawić dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, druki nr 985 i 1066. Wysoka Izbo! W trakcie drugiego czytania w dniu 14 kwietnia tego roku złożono do projektu ustawy 43 poprawki. Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia tego roku rekomenduje Wysokiej Izbie: odrzucić wniosek o odrzucenie ustawy, przyjąć poprawkę 28. oraz poprawki 37. i 39., poddane pod głosowanie łącznie, a także odrzucić wszystkie pozostałe poprawki i, co oczywiste, przyjąć projekt ustawy zawarty w sprawozdaniu komisji. Bardzo dziękuję. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1066. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawki. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Komisja wnosi o odrzucenie tego wniosku. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce podnieść rękę i nacisnąć

Sejm wniosek odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosowało 449 posłów. Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 11. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 14. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 15. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 16. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 17. poprawce wnioskodawcy proponują skreślić rozdział 5. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawek od 18. do 20. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 17. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 18. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

37 - za, 407 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 35. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 34. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pan i panów posłów jest za przyjęciem 35. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Nad nimi głosować będziemy łącznie. Głosujemy.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 38. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 40. poprawce do załącznika do ustawy - wzoru prospektu informacyjnego na s. 62 wnioskodawcy proponują zmianę w części III w rozdziale „Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym” Poprawkę tę rozpatrzymy łącznie z poprawką 43. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosownia nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1066, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Teraz będzie takie 5-minutowe głosowanie, więc jeśli państwo chcecie z tego skorzystać, to proszę. Będzie trwało 5 minut. Zamiast przerwy, panie pośle.

Sejm uchwalił ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Powracamy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1067- Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Marka Asta o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam przyjemność przedstawić dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1067-A i 1016. Komisja rozpatrzyła w dniu 15 kwietnia poprawki zgłoszone w drugim czytaniu. Dziewięć tych poprawek było.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1067. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Poprawki od 4. do 7. zgłoszone zostały do art. 2 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy - Prawo upadłościowe. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1067, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Wysoka Izbo! Jest to wniosek formalny o przerwę i rozszerzenie porządku obrad. Rzecz dotyczy kwestii, w której zdanie, jak sądzę, w tej Izbie podzielamy wszyscy: fakty, sprawy, które zaszły od wczoraj, poważnie godzą w bezpieczeństwo naszego kraju, a także godzą w bezpieczeństwo naszych sojuszników. Zaproponowaliśmy projekt uchwały, który jest już złożony, jest już u pani marszałek. Ze względu na solidarność międzynarodową, ze względu na bezpieczeństwo Polski, ze względu na poszanowanie prawa międzynarodowego uprzejmie proszę panią marszałek i państwa o to, żebyśmy rozszerzyli porządek obrad o punkt dotyczący uchwały, która wzywa rządy państw Unii Europejskiej i instytucje europejskie, szczególnie rząd Republiki Federalnej Niemiec, do zrobienia wszystkiego, co można zrobić na tym etapie, żeby zablokować budowę gazociągu Nord Stream 2.

Chwileczkę, nie skończyłam. Oprócz tego, że mogę przegłosować przerwę, natomiast drugiej części nie, panie pośle. Proszę państwa, ponieważ padł wniosek formalny o przerwę, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za ogłoszeniem przerwy, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Wszystko działa, pani poseł.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 25. porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały. Komisja wnosi o uchwalenie projektu uchwały z druku nr 974. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały z druku nr 974, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm podjął uchwałę w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej) Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 31. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1112 i 1115) Proszę pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie! W imieniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przedstawiam sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, druk nr 1115, o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1112. Marszałek Sejmu skierowała w dniu 16 kwietnia uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu rozpatrzenia. Senat zgłosił osiem poprawek. Niektóre zmniejszają wymiar i częstotliwość obowiązków nakładanych na właścicieli lub zarządców budynków, jest część poprawek redakcyjnych i legislacyjnych.

Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. Senat zgłosił do art. 1 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o efektywności energetycznej. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Senat proponuje, aby jednostka sektora publicznego informowała o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej i w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 6. i 7., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 8. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 32. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (druki nr 1113 i 1116) Proszę pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie! W imieniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przedstawiam sprawozdanie, druk nr 1116, Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, druk sejmowy nr 1113. Marszałek Sejmu skierowała w dniu 16 kwietnia 2021 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu rozpatrzenia. Senat zgłosił 15 poprawek. Komisja po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia wnosi, aby 12 poprawek przyjąć i 3 poprawki odrzucić.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Poprawkę tę rozpatrzymy łącznie z poprawkami 9. i 15. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 8., 9. i 15., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki 14., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 28. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Ale zanim przystąpimy do tego punktu, ogłaszam 5 minut przerwy.

obrady. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Nikt się nie zgłasza. Jako pierwsza z oświadczeniem - pani poseł Anna Dąbrowska-Banaszek. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

Reprezentuje on najliczniejszą, ponad 338-tysięczną grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne, w tym 299 tys. pielęgniarek i 39 tys. położnych. Według definicji z encyklopedii pielęgniarka w rozumieniu prawa polskiego - zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę: pielęgniarz - to samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje profesjonalną opiekę medyczną nad pacjentem. W ramach nabytych kompetencji pielęgniarka rozpoznaje warunki i potrzeby zdrowotne, diagnozuje problemy pielęgnacyjne pacjenta, sprawuje profesjonalną opiekę medyczną, realizuje zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, samodzielnie udziela określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych oraz prowadzi edukację zdrowotną. Obecnie w celu uzyskania uprawnień pielęgniarki należy posiadać minimum wykształcenie wyższe I stopnia, czyli licencjat pielęgniarstwa. Taka jest definicja. A życie? Działalność każdego podmiotu leczniczego, czy to w lecznictwie otwartym, czy zamkniętym, to wspólna, zespołowa praca wielu, w tym pielęgniarek i położnych. Chciałabym podziękować moim koleżankom i kolegom, pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym, za codziennie podejmowany trud, za wspólną pracę przez wiele lat. Dziękuję ci, Basiu, Agato, Ulu, Małgosiu, pani Mario, Jolu, Ewo. Dziękuję, Gerardzie. Dziękuję też wszystkim niewymienionym z imienia za pracę w dni powszednie, niedziele i święta, za trwanie na posterunku, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii. W 30. rocznicę waszego samorządu życzę wam dużo sił, satysfakcji z wykonywanej pracy, empatii wobec pacjentów i dużo zdrowia. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewicy. Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie! Szanowni Panowie! Z siedziby Sejmu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej mam zaszczyt przekazać państwu serdeczne zaproszenie do królewskiej Bydgoszczy, gdzie 2 maja o godz. 15 odbędzie się koncert patriotyczny zatytułowany „Pod biało-czerwoną” Koncert dedykowany jest naszej ojczyźnie z okazji jej doniosłych świąt majowych. Tym, co spaja nas i naszą ojczyznę, jest polska flaga, która towarzyszy nam w dniach radości i dumy, pod którą wszyscy czujemy się jedną wielką polską rodziną. Dlatego nasz koncert „Pod biało-czerwoną” będzie transmitowany na całą Polskę i na cały świat przez łącza internetowe. W bydgoskim koncercie wystąpią znani i lubiani artyści: Joanna Wojnowska i Krzysztof Filasiński, którzy zaprezentują państwu bogaty program zawierający polskie pieśni patriotyczne i operowe. Organizatorem koncertu jest znana działaczka społeczna pani Bogumiła Miler, prowadząca butik Oliwia. Firma butik Oliwia przeprowadzi także na żywo transmisję tego koncertu. Szanowni Państwo! Dla mnie jako posła ziemi bydgoskiej zaszczytem jest objęcie honorowego patronatu nad koncertem, który odbędzie się w Dniu Flagi Rzeczypospolitej. Wiemy, że koncert będzie wspaniałym patriotycznym i artystycznym przeżyciem. Dlatego raz jeszcze zapraszam panie i panów, wasze rodziny i waszych przyjaciół na koncert pod nazwą „Pod biało-czerwoną”, który od godz. 15 w dniu 2 maja będzie można obejrzeć na profilu facebookowym bydgoskiego butiku Oliwia.

Wierzymy, że niebawem będziemy mogli spotkać się osobiście. Panie i Panowie! Panie i Panowie! Zapraszamy do Bydgoszczy.

Panie Przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego Kaczyński! Panie Marszałku!

Od 2 lat TVP wmawia ludziom, że to moje słowa. Tymczasem są to cytaty, komentarze pod moimi postami, komentarze, które przytoczyłam, żeby pokazać, jak okrutni jesteście wy, wyznawcy kultu Kaczyńskiego. Każdy dzień rozpoczynam od takiego wylewu miłości bliźniego. A im więcej barw narodowych w zdjęciu profilowym, tym więcej inwektyw w komentarzach. To wy, drogie Polki i Polacy, i to wasze słowa, ale tym, kto je promuje i powiela w sieci, a potem zalewa nimi profile przeciwników politycznych, jest polski rząd, którego tutaj teraz nie ma. Ostatnie śledztwo niezależnych mediów dotarło do armii trolli na usługach partii rządzącej. To pokazuje, że PiS nas dzieli, skłóca, a w końcu stara się nas zniszczyć. Co więcej, robią to za publiczne pieniądze. Tak pokierowali milionami z państwowych spółek obsadzonych przez klany Dudów, Obajtków i Szydłów, że to my, podatnicy, płacimy za tych PiS-owskich hejterów. Jak mówił inżynier Mamoń: No i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, społeczeństwo. A na koniec chciałam się zwrócić na Wschód, tam, gdzie z niepokojem patrzą teraz obywatele wolnego świata: Putin, uwolnij Nawalnego. Poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska. Wysoka Izbo! Trochę historii. W maju 1867 r. zatwierdzono nowy projekt techniczny rozbudowy portu w Darłowie. Zakładał wtedy budowę portu o powierzchni 4,33 ha, budowę drugiego basenu wewnętrznego położonego naprzeciwko basenu zimowego, na prawym brzegu Wieprzy, budowę mostu stałego z portowymi basenami i likwidację mostu zwodzonego.

Budowa zachodniego falochronu spowodowała zwiększenie szerokości plaży zachodniej i przesunięcie linii brzegowej o ok. 100 m w morze. Rozbudowę portu umożliwiła ściągnięta z Francji w 1870 r. kontrybucja.

100 lat, szanowni państwo, a one już mają 139.

Nie chciałbym, szanowni państwo, żebyśmy się obudzili wtedy, kiedy coś się stanie. Dlatego dzisiaj proszę, panie ministrze infrastruktury, znajdźmy środki na projekt, znajdźmy środki na inwestycje, bo ten port jest dla Pomorza Zachodniego bardzo ważny nie tylko ze względu na rybaków i osoby pracujące, ale również ze względu na turystykę i bezpieczeństwo tego miasta. Bardzo o to proszę. Dziękuję bardzo. Poseł Konrad Berkowicz, koło Konfederacja. Pani poseł Wanda Nowicka, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Składam ogromne wyrazy ubolewania, że na oczach całego świata umiera Aleksiej Nawalny - wybitny opozycjonista, symbol walki o demokratyczną Rosję i prawa człowieka. Tymczasem demokratyczny świat temu się biernie przygląda. W prasie międzynarodowej można wiele przeczytać o Nawalnym, ale z tego kompletnie nic nie wynika. Żadne istotne decyzje nie zapadają. Potrzebna jest szybka i stanowcza reakcja, w tym nałożenie sankcji na Putina i Rosję. Wzywam, żeby polski rząd zrobił wszystko, by Unia Europejska i inne gremia międzynarodowe podjęły zdecydowane kroki dla ratowania Nawalnego. Trzeba działać teraz, a nie wtedy, kiedy będzie już za późno i nie będzie kogo ratować. Choć Rosja wydała na Nawalnego wyrok śmierci, i to nie raz, jeszcze możemy coś zrobić. Uratujmy Nawalnego.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 14 kwietnia obchodziliśmy Święto Chrztu Polski. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski i polskiego Kościoła katolickiego. Jednakże znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I nie ogranicza się tylko do jego osoby.

Chrzest Polski miał przełomowe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Wprowadzał państwo polskie w krąg krajów Europy Zachodniej. Nasza kultura, historia i tradycja oparte są na fundamencie tradycji chrześcijańskiej. Dziękuję wszystkim Polkom i Polakom za uczestnictwo w akcji „Wywieś flagę” z okazji tej wielkiej rocznicy. Dziękuję bardzo. Pani poseł Joanna Borowiak, klub Prawo i Sprawiedliwość. Wysoki Sejmie! Dziś ogłoszono bardzo dobrą informację dla mojego miasta Włocławka i dla mojego regionu. Rusza tak bardzo oczekiwana przez mieszkańców i podróżnych budowa dworca PKP. Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę z wykonawcą inwestycji, firmą Budimex SA. Jako poseł ziemi włocławskiej wyrażam swoją radość z tego, że został podjęty kolejny krok na drodze do realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji. Dworzec, który powstanie, zapewni komfort podróżnym, a także znacząco zmieni obraz architektoniczny miasta. Inwestycja została wpisana do „Programu inwestycji dworcowych” w 2017 r. i jest odpowiedzią na wieloletnie oczekiwania włocławian oraz podróżnych korzystających z usług PKP.

Dziękuję panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi za wpisanie modernizacji włocławskiego dworca do „Programu inwestycji dworcowych”

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

To bardzo piękna gmina, która, jak większość gmin w Polsce, ma swoje zasadnicze potrzeby.

Mieszkańcy Starego Zawidowa i wsi Wielichów nie mają bieżącej wody.

O to będę apelował.

Bardzo dziękuję. Pan poseł Konrad Berkowicz, koło Konfederacja. Każdy dorosły człowiek powinien być wolny. Co to znaczy: być wolny?

Na tym polega dorosłość. Na tym to polega. Jeśli ktoś jest dzieckiem, nazywamy go dzieckiem.

Taka jest zasada wolności. Dorosły człowiek za posiadanie czegoś takiego jest zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Dziękuję bardzo. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Na tym kończymy 28. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.